marszałków Sejmu i Senatu ubiegłych kadencji, [[Oklaski]] korpus dyplomatyczny wraz z jego dziekanem nuncjuszem apostolskim w Polsce Salvatore Pennacchio. Witam duchowieństwo z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski Jego Eminencją księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim. Witam członków Polskiej Rady Ekumenicznej oraz wszystkich przedstawicieli innych Kościołów i związków wyznaniowych. Witam dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z szefem Sztabu Generalnego generałem Rajmundem Andrzejczakiem.

Witam wszystkie panie i panów wybranych na posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich gości, którzy swoją obecnością uświetniają inaugurację 1. posiedzenia Sejmu IX kadencji. Szanowni Państwo! W dniu 8 listopada zmarł Stefan Strzałkowski, nauczyciel, samorządowiec, burmistrz Białogardu, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji.

Panowie Posłowie! Wielce Szanowny Panie Premierze! Szanowni Państwo Ministrowie! Dziekanie korpusu dyplomatycznego wraz ze wszystkimi ekscelencjami, przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, ambasadorami, konsulami i wszystkimi naszymi zagranicznymi gośćmi reprezentującymi swoje kraje w Rzeczypospolitej Polskiej! Eminencje, Ekscelencje, Księża Arcybiskupi i Biskupi! Wszystkie Osoby Stanu Duchownego obecne na tej sali i słuchające tego wystąpienia! Wszyscy Dostojni Przybyli Goście! Przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych! Wszyscy Wielce Szanowni Państwo! Jest to dla mnie niezwykły zaszczyt móc otwierać dzisiaj wraz z Państwem to pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji, Sejmu wolnej, niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej. W okresie szczególnym, tuż po 11 listopada, tuż po obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w tamtym pamiętnym 1918 r., ale także w roku szczególnym 2019, będącym zarazem Rokiem Powstań Śląskich, albowiem przypada w tym roku także I powstania śląskiego, będącym także rokiem 80-lecia wybuchu II wojny światowej, która tak mocno odcisnęła się na naszej historii - sama i to wszystko, co po niej nastąpiło - roku także i 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, a więc roku rocznic bardzo ważnych dla całego naszego społeczeństwa, dla wszystkich Polaków, żyjących nie tylko tutaj, w kraju, ale i na całym świecie, dla których bardzo często te wydarzenia były właśnie determinantą ich życiowych losów - bardzo często nie wyborów, tylko konieczności, które nimi w różny sposób pokierowały - i którzy dzisiaj także patrzą na nas i patrzą na naszą odpowiedzialność za dalsze losy Rzeczypospolitej. Ale z tego właśnie punktu widzenia chcę bardzo mocno podkreślić, że ta rozpoczynająca się IX kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tej właśnie wolnej, suwerennej i niepodległej po 1989 r., jest także i z całą pewnością niezwykłym czasem dla Państwa Posłów, dla Państwa najbliższych, bo jest to, jakkolwiek by na to spojrzeć, wielki zaszczyt móc z wyboru polskiego społeczeństwa, naszych wyborców, zasiadać w tej Izbie, dyskutować o najważniejszych polskich sprawach, dyskutować o tym, w jaki sposób powinna rozwijać się Polska, wymieniać się poglądami, reprezentując różne prądy ideologiczne, różne punkty widzenia na Polskę, ale Polskę, wobec której - nie mam żadnych wątpliwości - wszyscy byśmy chcieli, aby była Polską wolną, suwerenną i niepodległą po wsze czasy.

Za to wszystkim Polakom, i w kraju, i za granicą, wszystkim, którzy oddali swój głos, wszystkim, którzy zrobili to właśnie w poczuciu odpowiedzialności za sprawy naszego państwa, w poczuciu odpowiedzialności za naszą przyszłość, chciałem z całego serca podziękować. Dla wielu z nich był to wysiłek, także czasowy, zwłaszcza poza granicami, aby ten głos oddać. I chcę powiedzieć tak: bardzo mocno to doceniam i jestem przekonany, że bardzo wielu ludzi czujących odpowiedzialność i biorących dzisiaj tę odpowiedzialność za polskie sprawy na swoje barki również jest Państwu ogromnie wdzięcznych za ten właśnie wielki akt obywatelski.

Również apelowałem o frekwencję, bo uważam, że w istotnym stopniu jest to odpowiedzialność głowy państwa - aby namawiać, aby prosić rodaków, by tę odpowiedzialność za państwowe sprawy na siebie brali. Wiedzą Państwo doskonale, że to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności, to jest kwestia także tego, jaka będzie jakość legitymacji tych, którzy zostaną wybrani. Im wyższa frekwencja, tym legitymacja ta jest silniejsza, tym mocniejsze są organy o charakterze ustawodawczym czy prawodawczym, które oni reprezentują, myślę tutaj o Parlamencie Europejskim, myślę o polskim Sejmie, myślę o polskim Senacie. Trzeba powiedzieć jasno, że w tym roku, w roku 2019, Polacy zdali doskonale swój egzamin wyborczy, idąc gremialnie zarówno do wyborów europejskich, jak i do wyborów parlamentarnych. Z całego serca za to dziękuję.

Wyborcy na mnie zagłosowali. Jeszcze jeden element jest bardzo ważny, i to też z całą mocą chcę podkreślić. W ostatnich wyborach do Sejmu wynik był taki, że wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze mają dzisiaj swoich posłów w tej Izbie. Z mojego punktu widzenia jest to niezwykle ważne, bo to oznacza, że prawie wszyscy obywatele, którzy wzięli udział w wyborach, mają tutaj swoich reprezentantów, że są na tej sali osoby, które reprezentują ich punkt widzenia, z którymi oni zgadzali się w czasie kampanii wyborczej, słuchając ich wizji dotyczącej dalszego rozwoju Polski, słuchając, w jaki sposób chcą prowadzić politykę, do czego dążą i jakiej przyszłości dla naszego kraju oczekują. Jeszcze raz dziękuję z całego serca wszystkim moim rodakom za ten wspaniały, wielki sprawdzian odpowiedzialności za losy państwa, za ten wspaniały, wielki sprawdzian demokracji, jaki w Polsce się odbył i został zdany, rzeczywiście na bardzo pozytywną ocenę. To także jest kwestia tego, w jaki sposób będziemy postrzegani poza granicami kraju, w jaki sposób będzie postrzegana jakość naszego ustroju, naszego państwa, ale również i naszego społeczeństwa jako tego społeczeństwa, które jest prawdziwie obywatelskie, jako tego społeczeństwa, które jest prawdziwie świadome, jako tego społeczeństwa, które dokonuje wyboru swoich władz. Z całego serca za to dziękuję.

Gratuluję wszystkim Panom Posłom zasiadającym w tych ławach. To jest piękna sprawa zostać wybranym przez obywateli do polskiego Sejmu. Wiedzą Państwo, że miałem ten zaszczyt i tę przyjemność zasiadać z wami tutaj i przez 3 lata dyskutować o ważnych polskich sprawach. Był to ten okres mojego życia i ten okres mojej służby dla Rzeczypospolitej, który wspominam niezwykle mile. Bardzo cenne jest dla mnie wspomnienie kontaktów, które miałem wtedy z Państwem, spraw, które razem załatwialiśmy, dyskusji, czasem żarliwych, politycznych, ale w których było tak wiele ładunku merytorycznego, w których było tak wiele dobrych głosów na temat tego, jak powinna wyglądać Polska. Chciałbym życzyć Państwu, żeby takie właśnie debaty, podobne do tych, w których ja kiedyś mogłem tutaj brać udział, toczyły się w polskim Sejmie nadal, żebyście Państwo spokojnie mogli tutaj dyskutować o ważnych dla Polski sprawach. Jestem przekonany, że w bardzo wielu ważnych sprawach da się znaleźć porozumienie i da się znaleźć wspólne zdanie, nawet jeżeli istnieją różnice poglądów. Z całą pewnością są na tej sali osoby, które potrafią prowadzić taką merytoryczną, idącą ku przodowi, ku przyszłości, ku pozytywnej przyszłości, debatę polityczną. Chciałem pogratulować i podziękować również Państwa najbliższym. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bycie czynnym politykiem, zwłaszcza na forum ogólnopolskim, oczywiście jest wielkim zaszczytem, niesie ze sobą szereg możliwości właśnie dyskutowania i współdecydowania o polskich sprawach, ale bardzo często wiążę się także ze sporami politycznymi, wiążę się także z różnego rodzaju aktywnością medialną czy aktywnością mediów, która nie zawsze jest dla naszych rodzin miła. Chciałem podziękować wszystkim Państwa najbliższym, gratulując im tego wyboru, który został wobec ich bliskich dokonany. Chciałem im podziękować za to, że znoszą to, że Państwo tą polityką się zajmują, bo jestem przekonany, że wszyscy się nią zajmują dla dobra Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, chciałem także podziękować za Państwa aktywność w kampanii wyborczej, kampanii, która, jak wszyscy wiemy, jest okresem trudnym w polityce, i to trudnym z wielu punktów widzenia - trudnym z uwagi na spór ideologiczny, trudnym z uwagi na spór polityczny, ale trudnym także z uwagi na spory, które toczą się wewnątrz list wyborczych, a więc czasem w łonie własnego ugrupowania bywają sytuacje trudne. Chcę bardzo mocno podkreślić: to także, a może właśnie przede wszystkim dzięki Państwa pracy frekwencja wyborcza w tych wyborach była tak wysoka. Bardzo za to dziękuję, że rozmawialiście z obywatelami, że mówiliście o swoich programach, że mówiliście o swoich wizjach Polski. To bardzo ważne dla budowania demokracji i poczucia odpowiedzialności obywatelskiej w naszym kraju. Można śmiało powiedzieć, że dobrze zrealizowaliście to dzieło. Chciałem podziękować także tym, których w tej Izbie nie ma, którym, mimo że kandydowali, nie udało się dostać do Sejmu, nie zostali wybrani.

Państwu też bardzo serdecznie chciałem podziękować za odpowiedzialną kampanię wyborczą. Ta frekwencja jest także Państwa zasługą. Chcę też podzielić się pewnym osobistym spostrzeżeniem. Wiem, że wielu z Państwa z trudem przyjmuje tę sytuację, że te emocje, które towarzyszyły kampanii wyborczej, te emocje, które towarzyszyły temu swoistemu wyścigowi do ław sejmowych, powodują, że wielu z Państwa teraz z żalem patrzy na otwarcie tych obrad, myśląc: tak niewiele brakowało, czasem kilkaset, czasem kilkadziesiąt głosów, a to ja dzisiaj zasiadałbym w tych ławach. Otóż powiem tak: kiedyś, w 2007 r., także i ja po raz pierwszy startowałem w wyborach do polskiego Sejmu. Też było mi bardzo przykro. Nie znalazłem się wtedy tutaj, ale moja droga życiowa i polityczna, moja droga służby Polsce potoczyła się inaczej. I wierzę w to, że dla wielu z Państwa, chociaż nie znaleźliście się tutaj dzisiaj, ta droga także będzie w przyszłości drogą służby dla Rzeczypospolitej. Tego Państwu życzę. Bo ważne jest, aby ludzie, którzy chcą się podjąć służby dla Polski, służby dla współobywateli, mogli to realizować. Zwłaszcza w dzisiejszych, bardzo często trudnych czasach, o czym już przed momentem wspominałem. Szanowni Państwo!

Przez pryzmat tej właśnie odpowiedzialności jesteście Państwo dzisiaj obserwowani i przez pryzmat tej właśnie odpowiedzialności będziecie obserwowani także w ostatnim dniu swojego posłowania w tej IX kadencji. Także i z tego punktu widzenia będziecie Państwo oceniani, jeżeli będziecie chcieli ubiegać się o reelekcję parlamentarną, jeżeli będziecie chcieli ponownie ubiegać się o mandat poselski.

Patrzył wtedy na nas, w 10 lat po tym, kiedy były te pierwsze półwolne jeszcze wybory do Sejmu, ale które głosami naszych rodaków wyprowadziły nas z poprzedniego ustroju i wprowadziły nas rzeczywiście do wolnej, suwerennej i niepodległej Polski. Wtedy, już po 10 latach, mając pewność, że ten parlament, do którego mówi, to jest parlament wybierany przez obywateli w wolnych, rzeczywiście suwerennych, sprawiedliwych i uczciwych wyborach i że to jest reprezentacja polskiego narodu, powiedział tak: miejsce, w którym się znajdujemy, skłania do głębokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem z daru odzyskanej wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego. Jakże te słowa są znaczące.

One są najważniejszym przekazem, jaki Ojciec Święty mógł dać ludziom sprawującym władzę w Polsce i zasiadającym w tej Izbie, ludziom, którzy decydują o losach współobywateli.

Ogromnie bym chciał, żebyście Państwo tutaj, w tej Izbie te właśnie sprawy umieli rozpoznać. Dzisiaj wolno mieć różne poglądy.

Ale proszę Państwa, mamy również wiele różnych wyznań w Polsce. Są ludzie, którzy deklarują się jako katolicy, są ludzie, którzy deklarują się jako wyznawcy prawosławia, są ludzie, którzy deklarują się jako protestanci, jako ewangelicy - są bardzo różne religie dzisiaj. Wróciła także do Polski religia mojżeszowa. Co jest jednak ważne? Otóż chcę Państwu przypomnieć czasy, kiedy ta wielość religijna w Polsce była jeszcze silniejsza niż dzisiaj, kiedy mówiło się, że Polska jest w ogóle państwem wielonarodowym. Ja na kwestię narodowości patrzę w sposób specyficzny. Dla mnie Polakiem jest każdy ten, kto ma Polskę w sercu, to jest dla mnie najważniejsze kryterium. Jeżeli ktoś mnie pyta o kwestię narodowości, jeżeli ktoś ma co do tego jakieś wątpliwości, zawsze mówię: idź na cmentarz. Idź na cmentarz żołnierzy poległych w 1920 r. w obronie Rzeczypospolitej przed bolszewicką nawałą, idź na cmentarz żołnierzy poległych w 1939 r., idź na cmentarz poległych w powstaniu warszawskim, na każdy inny cmentarz tych, którzy stawali w obronie Ojczyzny, tamtej II Rzeczypospolitej przede wszystkim. Zobaczysz na tych grobach najprzeróżniejsze znaki: polskich żydów, polskich katolików, polskich Tatarów, wyznawców religii muzułmańskich. Wszyscy oni walczyli za Polskę, bardzo często na ochotnika, bo mieli ją w sercu, byli Polakami, chociaż mieli różne pochodzenie.

To jest właśnie to jedno i to jest to, co wszystkich ich łączyło: nasza wspólna wielka tradycja, ponad 1050 lat istnienia państwa polskiego, wyrosłego na korzeniach chrześcijańskich, chrześcijaństwa, które przyjęliśmy z Zachodu, chrześcijaństwa, które przyszło do nas z Rzymu poprzez Czechy. To wiele kultur, które tutaj ze sobą się spotykały, na tej ziemi, bo ona jest szczególna, na przebiegu wielu dróg prowadzących z Azji do Europy i w różne strony europejskie. Tak właśnie kształtowało się nasze społeczeństwo. I to jest ważne, bo to jest właśnie nasza wielka tradycja wyrastająca na korzeniach chrześcijańskich, ale tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich innych, także tych, którzy mają odmienne poglądy religijne czy poglądy ideowe. Chcę to z całą mocą podkreślić. To jest wielka tolerancja i to jest właśnie wielka istota tej wspólnoty, tego, że wszyscy żyjemy w Polsce i nazywamy się Polakami. Dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego zwracam uwagę, Wysoka Izbo, wielce szanowny Panie Marszałku, że widzę w ostatnich latach wiele kryzysów na tym tle, widzę w ostatnich latach w różnych sferach - nie mówię, że tylko w Wysokiej Izbie, choć niestety także tutaj się zdarzają - takie wypowiedzi, które wielu ludzi w Polsce mogą ranić, które uderzają właśnie w te najgłębsze warstwy naszej tradycji, źródła naszego pochodzenia, w to wszytko, w czym wyrośliśmy i co - bardzo mocno chcę to podkreślić - przez wiele lat naszej ogromnie trudnej historii pozwalało nam przetrwać najczarniejsze momenty, kiedy byliśmy pod zaborami przez 123 lata, a niektórzy przez 146, [[Oklaski]] kiedy nas rusyfikowano, germanizowano, kiedy próbowano wydrzeć nam właśnie tę naszą tradycję, wydrzeć nam naszą mowę, wydrzeć nam nasze przekonania, usiłowano zrobić z naszych przodków innych ludzi, innej kultury, innego obyczaju, innej mentalności. To się nie udało właśnie dzięki temu, że te korzenie były tak silne i tak głębokie, i tak niezwykle szanowane, przede wszystkim w polskiej rodzinie. To dzięki polskiej rodzinie, dzięki polskiej inteligencji, ale także dzięki polskim księżom, dzięki Kościołowi ta tradycja przetrwała i ta tradycja przyniosła nas do wolnej, niepodległej i suwerennej Polski w tamtym 1918 r. i potem także i kolejnymi zrywami ludzi w okresie komunistycznego zniewolenia, gdy nie byliśmy państwem w pełni wolnym, suwerennym i niepodległym. Część z Państwa doskonale te czasy pamięta, albowiem uczestniczyliście Państwo w tym wielkim procesie i wiecie, że wtedy mimo różnych podglądów i przekonań można było być jednością, a przede wszystkim nawet ci, którzy byli niewierzący, w ogóle niewierzący, bo przecież byli tacy zawsze, szanowali to, co leży u fundamentów, i to, co jest oparciem dla naszej tradycji i dla naszej kultury. Szanowni Państwo! Przypomnę słowa sprzed 30 lat: Nie stoimy jako naród na straconych pozycjach, jeśli zdobędziemy się na wysiłek, cierpliwość i wolę działania. Miejmy ufność w duchowe i materialne siły narodu. Wierzę, że Bóg nam dopomoże, byśmy uczynili wielki krok na drodze, która przed nami się otwiera. Szanowni Państwo! Kto 30 lat temu to powiedział? Na pewno są na tej sali tacy, którzy pamiętają te słowa. Powiedział je pan premier Tadeusz Mazowiecki w swoim premierowskim exposé w 1989 r. jako pierwszy niekomunistyczny premier odradzającej się Polski. Człowiek, którego szanują ludzie o bardzo różnych dzisiaj poglądach.

Będziemy je oczywiście różnie oceniali, ale one się dokonały. Ale zwróćcie Państwo uwagę, do czego się odwoływał: Miejmy ufność w duchowe i materialne siły narodu. Szanowni Państwo! Miejmy ufność cały czas w duchowe i materialne siły narodu i szanujmy je, także i te duchowe, bo są one w sercach bardzo wielu Polaków, są one dla nich ważne. I kiedy one są podważane, kiedy one są deptane, kiedy one są poniewierane, bardzo wielu ludzi, także i tych niewierzących, ale właśnie ufających w te duchowe siły, bardzo to boli i budzi zgorszenie.

Proszę o język parlamentarny w debacie, proszę o taki język, który nie będzie obrażał i nie będzie nikogo urażał, [[Oklaski]] bo to jest bardzo ważne. Poglądy można mieć, proszę Państwa, poglądy można mieć i trzeba je mieć, bo jeżeli ktoś nie ma poglądów, to nie powinien tutaj zasiadać. Zasiadacie tu Państwo właśnie dlatego, że te poglądy macie. One są bardzo często bardzo wyraziste, one są bardzo często bardzo mocne i głębokie, niektórzy używają słowa: radykalne, ale ja proszę, żeby język debaty nie był radykalny, żeby język debaty był językiem szacunku. Apelowałem już o to i będę o to apelował w nieskończoność, bo jest to Polsce niezwykle potrzebne i jest to - jestem głęboko o tym przekonany - oczekiwane przez większość naszych rodaków, żeby debata sejmowa nie obrażała i nie budziła zgorszenia. O to bardzo Państwa proszę, żeby zachowania, które mają miejsce w Sejmie, były zachowaniami o charakterze twórczym, a nie zachowaniami o charakterze destrukcyjnym, żeby zachowania także nie gorszyły. Możecie być Państwo tego pewni. Ja naprawdę wiele rozmawiam z naszymi rodakami, bardzo często się z nimi spotykam. Uważam, że jest to niezwykle ważny element służby publicznej, także tej prezydenckiej. Nie muszę Państwu o tym mówić. Oczekują merytorycznej debaty, oczekują poważnego mówienia o ważnych dla nich sprawach. Nie oczekują tego, aby czyjekolwiek poglądy były przez innych deptane. To budzi zgorszenie. Proszę, żeby tego tutaj, w tej Izbie nie było. I chcę zaznaczyć bardzo wyraźnie jedno: coś, co już tutaj mówiłem do części z Państwa, bo część Państwa po raz pierwszy zasiada w tej Izbie, ale część - to są twarze znajome po wszystkich stronach sceny politycznej. Powiem tak, mówiłem to i będę zawsze powtarzał: Jestem przekonany, że wszyscy Państwo mimo różnic w poglądach zasiadacie tutaj z pobudek patriotycznych. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Chcę to z całą mocą podkreślić. Pewnie, że są emocje - tak jak powiedziałem, proszę, żeby starać się je powściągać - pewnie, że są dyskusje, ale nie mam wątpliwości, że w każdej z tych dyskusji jest Polska, różnie widziana, takie jest prawo wszystkich Państwa. Wyborcy wybierają, którą wizję w danym momencie uważają za słuszniejszą, za bliższą ich sercu, bliższą ich osobistym przekonaniom czy bliższą ich osobistym pragnieniom, bliższą temu, jak chcą, żeby się Polska rozwijała. Ale proszę, żeby to szanować, szanować w obie strony i szanować siebie nawzajem. Szanowni Państwo! Mówiłem już te słowa, ale powtórzę je jeszcze raz: Pan prezydent Lech Kaczyński, mój prezydent, prezydent, którego byłem kiedyś ministrem, co uważam za wielki zaszczyt, którego dostąpiłem w swoim życiu, powiedział, że podstawą patriotyzmu w odróżnieniu od nacjonalizmu i innych postaw jest miłość - miłość do Ojczyzny, ale także do drugiego człowieka, do współobywatela. Niech ona, proszę Państwa, będzie tym elementem podstawowym przed wszystkim, [[Oklaski]] także przed wszystkim, co się dzieje i o czym mówi się tutaj, w tej Izbie. O to proszę. To jest bardzo ważne także i dla jakości debaty, która będzie prowadzona tutaj przez najbliższe 4 lata. Szanowni Państwo! Na zakończenie chcę życzyć, żeby Państwo tutaj, służąc Rzeczypospolitej i naszym współobywatelom w tej Izbie, osiągnęli swoje cele i zrealizowali także swoje pragnienia. One są ważne. Ludzie o tym mówią. To jest bardzo ważne, żeby ludzie o Sejmie i o posłach mówili dobrze, że to są ludzie uczciwi, którzy rzeczywiście ciężko dla nich pracują. Bo ja wiem o tym, że w ogromnej, absolutnej większości przypadków tak właśnie jest, że Państwo bardzo ciężko pracują po to, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, dla swoich wyborców, dla Rzeczypospolitej. Oczywiście media w różny sposób to pokazują. Media interesują się tym, żeby coś się działo. Spokojna dyskusja nie służy zainteresowaniu, ale jest bardzo potrzebna, bo wtedy sprawy będą załatwiane merytorycznie, będą załatwiane dobrze. Tak, jak mówiliśmy, i tak, jak mówię, Polska jest jedna i proszę, żeby Państwo zawsze o tym pamiętali. Chciałbym, żebyście Państwo teraz, na rozpoczęcie tej kadencji, na początek podali sobie rękę, po prostu, tak zwyczajnie, jak ci, którzy spotykają się po to, żeby toczyć debatę o bardzo ważnych sprawach i umieją usiąść i spokojnie dyskutować, po to, żeby się spotkać i rozejść w pokoju i przyjaźni - mimo wszystkich różnic i podziałów.

Powinniśmy robić wszystko, żeby tych sporów, zwłaszcza wewnątrzrodzinnych, było jak najmniej. Czasem mówią: Ryba psuje się od głowy. Głowa jest tutaj. Dziękuję bardzo.

Panie Prezydencie! Bardzo dziękuję za obecność.

Witam, panie prezydencie. Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! Dostojni Goście! Inauguracja nowej kadencji Sejmu to zawsze moment szczególny. Moment, w którym jako przedstawiciele narodu stajemy przed naszymi współobywatelami i przed społecznością międzynarodową, której stanowimy część. Dlatego w pierwszym rzędzie chciałbym się odnieść do wszystkich Polek i wszystkich Polaków, do narodu polskiego, którego poświęcenie, wytrwałość i ofiarność doprowadziły w długim procesie po 1989 r. do odzyskania niepodległości.

Nie ma dziś wolności i demokracji poza niepodległością. Cytat ten pochodzi z tekstu napisanego w 1976 r. w środowisku harcerskim Pierwszej Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka” Program zawarty w tym tekście dał początek nowoczesnemu ruchowi niepodległościowemu, zbudował Komitet Obrony Robotników, odnalazł następnie swoją realizację w największym ruchu społecznym w dziejach współczesnego świata - w „Solidarności” To wielkie odrodzenie narodowe próbowano następnie złamać działaniami zbrojnej grupy przestępczej kierowanej przez aparat komunistyczny, wydając wojnę narodowi polskiemu w 1981 r. Zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana i nie wyciągnęliśmy konsekwencji wobec odpowiedzialnych. Stan wojenny to nie tylko setki zabitych, w tym księży zamordowanych podczas rozmów okrągłego stołu. To także tysiące więzionych, wyrzuconych z pracy i skazanych na emigrację. To przede wszystkim przygotowanie długofalowej struktury grabieży narodu polskiego, niszczenia jego gospodarki, wywłaszczenia z owoców jego pracy wielu, wielu pokoleń. To także ponowna próba wykreślenia z polskiej historii prawdy o okupacji sowieckiej, o bohaterskim zbrojnym oporze żołnierzy wyklętych, niezłomnych. To wreszcie haniebna chęć wykorzystywania Wojska Polskiego jako najemnych oddziałów okupacyjnych obcego mocarstwa. To smutne dziedzictwo wciąż nie zostało w pełni przekreślone i odrzucone. I chociaż w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne, niesłychanie istotne zmiany w sprawach społecznych, gospodarczych i historycznych, odpowiedzialność za ostateczne uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas, panie posłanki i panowie posłowie. Bo dzisiaj świadomość ograniczeń związanych z dziedzictwem - tamtym dziedzictwem - jest dużo głębsza niż wcześniej. To właśnie dlatego naród powierzył nam swój mandat. Mamy świadomość tej odpowiedzialności. Dziękujemy za to niezwykłe wyróżnienie i przyjmujemy ten obowiązek. Bez względu na różnice polityczne wszystkich nas musi łączyć miłość do ojczyzny i wola potępienia zbrodni przeciwko narodowi. Sejm IX kadencji jest do tych obowiązków przygotowany lepiej niż jakikolwiek inny, bo zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz, wybierając najbardziej reprezentatywny sejm czasów najnowszych. Żaden z dotychczasowych sejmów Rzeczypospolitej, począwszy od 1919 r., nie reprezentował takiej woli jedności narodowej jak ten, w którym dziś zasiadacie panie i panowie posłowie. Fenomenem jest masowy, ponad 60-procentowy udział Polaków w ostatnich wyborach. Ma to olbrzymie znaczenie dla przyszłości Polski i świadczy o niezwykle wysokiej świadomości obywatelskiej wyrastającej z przekonania, że państwo jest narzędziem realizacji woli narodu. Ta świadomość pokazuje skalę przemian, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 4 lat w naszej ojczyźnie, i jest to wynik działań obozu patriotycznego. Jego fundamentem jest głęboki demokratyzm Polaków odwołujący się do jednej z najstarszych i najtrwalszych w Europie tradycji demokratycznych. Sejmy piotrkowskie, konstytucja nihil novi, Trybunał Koronny - cała ta wspaniała tradycja demokracji szlacheckiej dzięki Konstytucji 3 maja, pracy organicznej ruchu narodowego i powstańczym dokonaniom żołnierzy, aż po żołnierzy niezłomnych i „Solidarność”, są spuścizną, do której z dumą dzisiaj nawiązujemy. Istotą tej tradycji są wolne wybory Sejmu, parlamentu Rzeczypospolitej. Nie przypadkiem rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, kierowany przez premiera Tomasza Arciszewskiego z Polskiej Partii Socjalistycznej, podjął w 1945 r. decyzję, że to wolne wybory do Sejmu będą niezbędnym świadectwem, iż Polska jest naprawdę niepodległa, i dopiero po ich przeprowadzeniu mogą zostać przekazane do kraju insygnia niepodległego państwa polskiego. Parlament jest najwyższą instytucją państwa polskiego stanowiącą prawo. To parlament wraz z prezydentem kształtuje prawa, instytucje i stosunki społeczne, bo tylko prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i parlament mają szczególny mandat narodu do decydowania o kształcie państwa polskiego. Ten autorytet i tę wolę demokratycznego państwa polskiego wszystkie pozostałe instytucje powinny respektować. Jest też druga istotna cecha obecnej kadencji Sejmu, o której trzeba powiedzieć. Chociaż reprezentując wszystkie nurty polityczne narodu polskiego, jest ten Sejm bardzo zróżnicowany, to absolutna większość wyborców wsparła te ugrupowania, które jednoznacznie odwoływały się do wartości narodowych, niepodległościowych, katolickich. Ukształtowanie naszych instytucji państwowych, życia gospodarczego i społecznego zgodnie z tymi wartościami to nasze największe zadanie, jakie stoi przed obecnym Sejmem. Polacy mają prawo oczekiwać, że ich wola zostanie uszanowana. Oczywiście odpowiedzialność spada przede wszystkim na większość rządową, bo po raz pierwszy w historii Polacy w tak zdecydowany sposób dali jednej formacji obowiązek utworzenia jednorodnego rządu. To wielkie zaufanie, takie, jakiego nie miał żaden rząd ani żaden przywódca w powojennej historii Polski. Ono musi zostać dotrzymane. Determinacja narodu wyrażona wynikiem wyborów nie jest przypadkiem, lecz skutkiem realizacji podstawowych zasad polityki niepodległościowej rozpoczętej jeszcze przez rząd śp. Jana Olszewskiego, a kontynuowanej później przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Przełomem było odrodzenie narodowe po roku 2010. Jego źródłem była wielka fala powrotu patriotyzmu, świadomości narodowej i polskich obowiązków, żywa zwłaszcza wśród młodzieży, która najgłębiej przeżyła dramat katastrofy smoleńskiej. Bez względu na opinie o przyczynach tej tragedii uświadomiła ona nam wszystkim, jak kruche były dotychczasowe przemiany, jak ważne jest silne państwo polskie i bezpieczeństwo militarne, a przede wszystkim, jak wielkie jest stale ciążące nad nami zagrożenie zewnętrzne. To właśnie tutaj miał swoje źródło program odbudowy silnej armii, reformy sądownictwa, reformy szkolnictwa. reformy socjalnej, a przede wszystkim dążenie, by przywrócić państwo narodowi. W zeszłej kadencji budowaliśmy fundamenty, często kwestionowane przez tych, którzy chcieliby zawrócić bieg historii. Domagano się likwidacji naszych najważniejszych osiągnięć gospodarczych, społecznych, tożsamościowych. Temu miały służyć żądania likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Wojsk Obrony Terytorialnej, sojuszu strategicznego ze Stanami Zjednoczonymi. pamięci o żołnierzach niezłomnych, suwerenności energetycznej, trwałości rodziny i wychowania opartego na wartościach chrześcijańskich. Był to program, który mógł być zrealizowany tylko w oparciu o siły zewnętrzne, o wzniecenie nienawiści i się do wszystkich pań posłanek i posłów o odrzucenie tej negacji niepodległego państwa polskiego i fundamentów cywilizacji chrześcijańskiej. Zwracam się o szacunek dla niepodległościowego wysiłku narodu polskiego, dla milionów ofiar okupacji niemieckiej i sowieckiej, dla utraconych szans przez tysiące odrzuconych, lekceważonych i pogardzanych. Przez ostatnie lata Polacy odzyskali poczucie godności własnej, siły narodowej, stali się wreszcie gospodarzami we własnym domu. To wartości bezcenne, które należy wzmacniać, a nie niszczyć. Czas więc zacząć wznosić gmach niepodległego państwa polskiego opartego na zasadach wywiedzionych z chrześcijańskiej nauki społecznej. Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem doskonale wiemy, jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy, jaką cenę płacimy za porozumienia okrągłego stołu, jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender. Wiemy, co oznacza pozostawienie środowisk agenturalnych na ważnych stanowiskach w administracji publicznej, [[Poruszenie na sali, oklaski]] na wyższych uczelniach, w wymiarze sprawiedliwości i w mediach. Wiemy też, jakie są zagrożenia geopolityczne wynikające z utopijnej próby budowania neosocjalistycznego imperium, kto jest naszym rzeczywistym sojusznikiem strategicznym. Wiemy wreszcie, że naród, który nie jest w stanie obronić swojej niepodległości i odbudować potencjału demograficznego, musi upaść. Wiemy więc, przed czym musimy się bronić i dokąd chcemy dojść. Musimy zbudować silne państwo narodowe z jasną hierarchią wartości odróżniającą patriotyzm od zdrady, dobro od zła, cywilizację życia od cywilizacji śmierci, równocześnie szanując demokrację i różnicę poglądów. Tego właśnie uczył nas bł. ks. Jerzy Popiełuszko, powtarzając za św. Pawłem: zło dobrem zwyciężaj. Wspólną płaszczyzną tej pracy jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy obywatele, a zwłaszcza ci, którzy stanowią prawo, muszą szanować ustawę zasadniczą.

Bardzo dziękuję, a teraz proszę zachować ciszę. Trzy artykuły konstytucji tworzą prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. Art. 8 gwarantuje niepodległość państwa polskiego poprzez stwierdzenie, że to właśnie konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Rola konstytucji jest szczególna, to ona jest w Polsce najwyższym prawem. Tak jest i tak musi pozostać. Konstytucję można naprawiać, zmieniać, ulepszać, ale dzisiaj stoi ona ponad wszystkimi różnymi źródłami prawa. Zresztą takie samo stanowisko sformułował Trybunał Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej w orzeczeniu z 11 maja 2005 r., a także w orzeczeniu z 24 listopada 2010 r. Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej chroni rodzinę rozumianą jako związek kobiety i mężczyzny.

Dziękuję bardzo za poparcie. Dokładnie ten przepis brzmi: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Żaden przepis nie jest ważniejszy dla umacniania demograficznego rozwoju narodu, wspierania jego spoistości i gwarantowania ładu oraz bezpieczeństwa społecznego.

Te trzy artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej tworzą, jak powiedziałem, prawną, społeczną i moralną podstawę naszego ładu państwowego. Jestem przekonany, że wszyscy posłowie bez względu na opcje polityczne zgodzą się współdziałać tu, w Sejmie, w oparciu o te właśnie zasady.

Nasza siła leży we współdziałaniu. Nasza siła wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej. Wreszcie naszą siłą jest gotowość poświęcenia życia dla niepodległości, bo niepodległość jest warunkiem podstawowym, sine qua non realizowania wszelkich wartości narodowych. Nie ma dzisiaj wolności i demokracji poza niepodległością. Niepodległość, panie posłanki i panowie posłowie, ma jeden kształt, wiele postaci ma niewola.

Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam niewątpliwy zaszczyt - jestem wzruszona - i wielką przyjemność rekomendować kandydaturę pani poseł, pani marszałek Elżbiety Witek na stanowisko marszałka Sejmu IX kadencji. Pełniąc ten urząd do tej pory, pani poseł, pani marszałek Elżbieta Witek wykazała się ogromną sprawnością organizacyjną, opanowaniem oraz wysoką kulturą osobistą.

Wymienię zaledwie kilka. Elżbieta Witek była ministrem, członkiem Rady Ministrów, szefem gabinetu politycznego premiera, a także rzecznikiem rządu. Od czerwca 2019 r. pełniła urząd ministra spraw wewnętrznych i administracji. W sierpniu 2019 r. pani poseł Elżbieta Witek została wybrana na marszałka Sejmu VIII kadencji. Podkreślę to: sprawując urząd marszałka Sejmu, udowodniła, że jest obdarzona ogromnymi zdolnościami organizacyjnymi, zdecydowana w działaniu, opanowana. Wysoka Izbo! Pani poseł, pani marszałek Elżbieta Witek jest doświadczonym parlamentarzystą.

Pracowała w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, Komisji Etyki Poselskiej, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a także Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Elżbieta Witek była lubianym przez uczniów nauczycielem, cenionym dyrektorem szkoły podstawowej, a także zespołu szkół ogólnokształcących w Jaworze.

Od 2001 r. jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, od 2011 r. - członkiem komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

Przy naszej koleżance, przyjaciółce Joli Szczypińskiej była do ostatniej chwili. Wysoka Izbo! Elżbieta Witek to pełnowymiarowy człowiek. Jest bardzo ceniona w swoim regionie, w swoim mieście nie tylko przez zwolenników politycznych. Wysoka Izbo!

Elu - pozwalam sobie tak powiedzieć, pozwolić na taką formę, bo znamy się od ponad 20 lat - wiem, że dasz radę utrzymać nas tu wszystkich w ryzach, a wszystko po to, żeby usprawnić prace Sejmu, który prawnie reguluje życie Polski i Polaków. Powodzenia, Elu. Bardzo dziękuję, pani poseł. Zanim przejdziemy do dalszej części procedury, chciałbym zapytać, czy wszyscy posłowie posiadają tymczasowe karty do głosowania.

W takim razie otwieram dyskusję. Proponuję, aby w dyskusji Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła poselskiego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę.

Wysoka Izbo! Koalicja Obywatelska szanuje zasady demokracji i reguły parlamentarne, Koalicja Obywatelska szanuje prawo większości sejmowej do zgłoszenia kandydata na marszałka Sejmu, dlatego też nie wystawiamy innej kandydatury i dlatego też nie będziemy głosować przeciwko tej kandydaturze. Jesteśmy przekonani, że to prawo większości w Izbie będzie tak samo szanowane przez państwa przedstawicieli w drugiej z Izb polskiego parlamentu, a mianowicie w Senacie. Jestem przekonany, że zasady parlamentaryzmu powinny przyświecać tej kadencji i tutaj powinniśmy odczuć bardzo dużą zmianę. Przypominam również, że przed nową marszałek Sejmu stoją bardzo ważne wyzwania i konieczność przestrzegania prawa. Przypomnę, że od nowego marszałka Sejmu oczekujemy niezwłocznego wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego [[Oklaski]] i upublicznienia list poparcia sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Od marszałka Sejmu oczekujemy również elementarnej przyzwoitości i niekarania posłów opozycji tylko dlatego, że w swoich wystąpieniach powiedzą o czymś, co nie spodoba się tym czy innym działaczom partyjnym. Od marszałka Sejmu oczekujemy wreszcie tego, by debata parlamentarna wróciła do tych elementarnych standardów, których tak bardzo brakowało w tym parlamencie pod rządami pani poprzednika. Raz jeszcze chcę podkreślić, że to będzie wielkie wyzwanie dla nowego marszałka, który nie słowami, a czynem będzie musiał udowodnić, co jest dla niego najwyższą wartością: przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o której państwo dzisiaj tak płomiennie mówili, czy też dyspozycje z tej czy innej centrali partyjnej. Ale przed nowym marszałkiem Sejmu będzie również kolejne wyzwanie, dotyczące odpowiedniego przygotowania oraz procedowania w tym parlamencie przepisów, które będą wykonywały ewentualne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo przypomnę, że w przyszłym tygodniu będą rozstrzygnięcia, które będą dotyczyły tego, czy Polska nadal będzie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, czy też - tak jak będą podpowiadać pani, pani marszałek, partyjni lub koalicyjni koledzy - ma stać na obrzeżach Unii Europejskiej, ślepo podążając w wytyczonym wcześniej bardzo złym kierunku dewastacji wymiaru sprawiedliwości. Liczymy, pani marszałek, że pani samodzielność i niezależność zostanie udowodniona w najbliższych dniach, a przede wszystkim, że wykona pani prawomocne wyroki sądowe. Z tego też względu, dając ten swego rodzaju kredyt zaufania, szanując reguły parlamentaryzmu, licząc na szacunek dla tych reguł w drugiej Izbie, czyli w Senacie, nie będziemy głosować przeciwko pani kandydaturze. Głos ma poseł Krzysztof Gawkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Lewica wróciła do polskiego parlamentu. Lewica mądra i rozsądna. Lewica, która ma poczucie szacunku do konstytucji, szacunku do tego najważniejszego aktu prawnego, dlatego nie zgłosi kandydata na marszałka Sejmu, ale w poczuciu odpowiedzialności, że można być opozycją mądrą i rozsądną, szukającą porozumienia, godności, szacunku dla człowieka, szacunku dla wartości, poprzemy kandydaturę pani marszałek Witek na stanowisko marszałka Sejmu. Chcemy poszukiwać odpowiedzialności za słowa i za czyny, dlatego przez najbliższe 4 lata będziemy się przyglądali, jak pani marszałek będzie realizowała te konstytucyjne obowiązki, które zostaną na panią dzisiaj nałożone. Chcemy, żeby Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej była wyznacznikiem poczucia współpracy pomiędzy partiami, ale i osobami, które dzisiaj zasiadły w polskim parlamencie. Zwracamy się zatem do pani marszałek z apelem, który kierujemy jeszcze przed oficjalnym wyborem, ale w poczuciu, że ten wybór pewnie nastąpi. Przedstawiciele Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy uważają, że powinniśmy zaczynać pierwsze posiedzenie Sejmu od rzeczy fundamentalnych, które będą pokazywały, że jesteśmy Sejmem otwartym na społeczeństwo, od którego 2016 r. zostaliśmy odgrodzeni haniebnymi barierkami. IX kadencja Sejmu może zacząć się właśnie od takiego symbolicznego otwarcia w zakresie i dyskusji, i wymiany poglądów, ale i otwarcia Sejmu, zdjęcia tych barierek. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Współpraca to wola porozumienia, współpraca to szacunek dla godności, dla wartości, które wyznajemy. Lewica, która w wyborach parlamentarnych wiele razy mówiła o tym, że chcemy być tą częścią opozycji, która nie będzie recenzowała bez pokazywania przykładów, jak niedobre dobrym zastępować, będzie w tej kadencji również szukała porozumienia w sprawach społecznych, socjalnych, odpowiedzialności za państwo, poczucia, że demokracja nie jest tylko w słowach, ale też w czynach i w gestach, i w głosowaniach na tej sali sejmowej. Oczekujemy, że taka współpraca będzie również ze strony pani marszałek. W polskim parlamencie w IX kadencji zasiadają różne frakcje polityczne. Te różne frakcje polityczne powinny mieć szacunek do konstytucji, ale i do tego, co będzie tutaj padało. Chciałbym zagwarantować w imieniu naszego klubu, że głosując dzisiaj za panią marszałek, udzielamy tego swoistego wotum zaufania, że możemy razem rozmawiać o Polsce, w trosce o Polskę, że razem możemy doprowadzić do sytuacji, w której polski Sejm będzie nazywany kuźnią idei, a nie kuźnią, w której łamiemy demokrację. Dziękuję panu posłowi. Głos zabierze teraz pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja.

Głos zabierze pan poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Panie Prezydencie! Panie Premierze! Wysoka Izbo!

Moi drodzy, szanowni państwo, polski parlamentaryzm, debata parlamentarna wymaga odrodzenia. Ten dzisiejszy dzień jest takim dobrym początkiem, który daje szanse na odrodzenie dobrych zasad, zwyczajów, obyczajów, kultury zabierania głosu. Pan prezydent Andrzej Duda mówił o tym w swoim wystąpieniu, szanując wszystkie strony sporu politycznego, szanując wszystkich, którzy zasiadają w Wysokiej Izbie, i dziękując milionom naszych rodaków, którzy oddali na nas głos. Ten szacunek powinien być nie odświętny, tylko codzienny. Ten szacunek jest naszym zobowiązaniem wobec tych wszystkich, którzy głosowali na nas, ale również na naszych konkurentów. Dlatego w imieniu klubu parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz’15 z szacunkiem odnosimy się do werdyktu wyborczego, w którym partia Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory i ma prawo zgłosić kandydata na marszałka Sejmu, ma prawo utworzyć rząd i ma taki obowiązek, bo to jest zobowiązanie. Dlatego, szanując ten werdykt wyborczy, wierząc, że jest możliwa lepsza debata parlamentarna, jest możliwa lepsza dyskusja, przez to jest możliwa lepsza Polska dla nas wszystkich, dla naszych rodaków, poprzemy kandydaturę pani marszałek Witek.

Liczymy na debatę, liczymy na rozpatrzenie naszych projektów. W pierwszych 100 dniach zgłosimy projekty dotyczące emerytury bez podatku, dotyczące pakietu obywatelskiego Pawła Kukiza, sędziów pokoju, dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych czy podniesienia kwoty wolnej od podatku, zgłosimy projekty dotyczące dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, dotyczące zerowego VAT-u na zdrową żywność i chcielibyśmy, żeby te projekt nie leżały w zamrażarce, tylko były rozpatrzone, ale nie tylko rozpatrzone, ale też żeby była wykonywana nad nimi realna praca. Dzisiaj jest kredyt zaufania. Cieszę się, że inne kluby parlamentarne: Lewica, ale też takie może jeszcze nie poparcie, ale życzliwe podejście Koalicji Obywatelskiej, Platformy. To pokazuje, że w tym zwariowanym świecie animozji politycznych może być trochę normalności. Pewnie jeszcze więcej by jej było, gdyby projekt, który PiS zgłaszał, będąc w opozycji, pakiet demokratyczny, był przyjęty, kiedy rządzi. Jest taka możliwość.

Będziemy rozliczani z posunięć politycznych.

Pani Marszałek!

Raz jeszcze przepraszam za pomyłkę.

Bardzo proszę. Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo! W ciągu ostatnich lat obserwowaliśmy proces zaostrzania się debaty publicznej. Widzimy proces polaryzacji debaty publicznej, a przede wszystkim proces wykluczania z debaty publicznej.

Skończyło się tylko na wyrzuceniu z sali konferencyjnej.

Podczas debaty wyborczej, zwłaszcza w mediach publicznych, Konfederacja była całkowicie wykluczana. Dlatego chcieliśmy skorzystać z okazji i zadać pani kandydat, pani marszałek pytanie. Prosimy o ustosunkowanie się do niego, bo od tego będzie zależało to, jak Konfederacja zagłosuje nad pani kandydaturą na fotel marszałka. Dzisiaj wybieramy nie tylko marszałka Sejmu, lecz także prawdopodobnie całe Prezydium Sejmu. Mam do pani marszałek pytanie.

Od tego uzależniamy naszą decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Najpierw chciałem pogratulować wystąpienia panu marszałkowi seniorowi.

Tak, będziemy to robić, ponieważ, szanowni państwo, tego dzisiaj wymaga polska racja stanu.

Chcielibyśmy, żeby debata, która będzie się toczyć na sali plenarnej, była również debatą, podczas której nie będzie mrożenia ustaw, tak jak było w poprzedniej kadencji np. w przypadku ustawy o bratniej pomocy.

Tego oczekujemy od tego Sejmu, od tej nowej kadencji.

Wkraczamy do tego Sejmu z tą agendą, z tym programem. Bardzo dziękuję, panie pośle. Czy ktoś jeszcze pragnie zabrać głos? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! Naprawdę z wielką radością wysłuchałem oświadczeń partii, a także koła, chociaż tutaj mieliśmy do czynienia z pewną różnicą, i podsumowałbym to tak: koniec opozycji totalnej. Jeśli tak rzeczywiście będzie, to będzie to naprawdę wielki postęp w naszym życiu publicznym i zmiana, której z całą pewnością oczekuje społeczeństwo, zmiana w interesie polskiej demokracji, polskiego społeczeństwa, polskiego narodu, polskiej przyszłości. Tak że bardzo, bardzo proszę o to, żeby to nie były tylko słowa, żeby to były także czyny, również tutaj, w tej Izbie. Ale jednocześnie te wystąpienia zawierały także pewne elementy, z którymi się nie można zgodzić. Chodzi o pewne elementy, które można by określić jako reprymendę, strofowanie. Otóż my w tym wypadku podtrzymujemy nasze zdanie i podtrzymujemy także inne zdanie, które chyba też musi tutaj paść. Większość ma prawo powołać rząd, ma oczywiście prawo powołać marszałka, ale większość ma także prawo rządzić, tzn. realizować swoją agendę, oczywiście w dyskusji, w kulturalnej, merytorycznej dyskusji i przyjmując merytoryczne argumenty innych. To jest oczywiste. Oczywiste jest także to, o czym też muszę wspomnieć, że klubem, który ma najwięcej swoich reprezentantów w wyższej Izbie naszego parlamentu, czyli w Senacie, jest Prawo i Sprawiedliwość i z tego też muszą być wyciągnięte pewne wnioski. W każdym razie nie będę jednak słuchał tego, co tutaj znów pada i co mi przypomina tamte obrady. Miejmy nadzieję, że to przejdzie do historii. Bardzo, bardzo dziękuję za to, że tak rozpoczyna się ta kadencja Sejmu.

Bardzo dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Wysoka Izbo! Sejm, zgodnie z art. 4 ust. 3 regulaminu Sejmu, wybiera marszałka Sejmu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kto z państwa jest za kandydaturą pani poseł Elżbiety Witek, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Sejm bezwzględną większością głosów wybrał panią poseł Elżbietę Witek na stanowisko marszałka Sejmu.

Bardzo proszę panią marszałek o zajęcie miejsca.

Jesteśmy pod wrażeniem tak szerokiego poparcia dla pani marszałek

To jest wyjątkowy dzień dla mnie, ale myślę, że też wyjątkowy dzień w tej Izbie.

To jest dla mnie ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie i oczywiście zobowiązanie.

Myślę, że kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że w 37-milionowym narodzie jest 460 takich, którzy decydują o najważniejszych sprawach dla naszej ojczyzny i dla naszych obywateli, to jest to naprawdę ogromne wyróżnienie, że zasiadamy tutaj, w tej Izbie. Chciałam bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi seniorowi za sprawne przeprowadzenie pierwszej części naszych obrad. Dziękuję bardzo.

Jako marszałek Sejmu będę robiła wszystko, żeby każdy z państwa znalazł u mnie wsparcie, wtedy kiedy tego wsparcia będziecie państwo potrzebowali, zgodnie z regulaminem Sejmu. Drzwi do mojego gabinetu będą dla państwa otwarte. Jak mówią, z każdej sytuacji są co najmniej dwa wyjścia, będziemy starali się poszukiwać tego najlepszego. Oczywiście dziękuję władzom mojego klubu i mojej partii za to, że wysunęły moją kandydaturę na to stanowisko. Mam nadzieję, że nie zawiodę nikogo.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Nitras z wnioskiem formalnym? Serdecznie dziękuję.

Od rana czytamy, słyszymy informacje, że większość ma zamiar ogłosić przerwę bez wybierania Prezydium Sejmu, w oczekiwaniu na rozstrzygnięcia w innej Izbie. Jeżeli ta atmosfera jest taka dobra, jeżeli wszyscy zgadzamy się z tym, że można w tej atmosferze pracować, to apelujemy: nie róbmy żadnej przerwy, tylko wybierajmy Prezydium Sejmu, tak jak to przewiduje porządek obrad tego posiedzenia, korzystajmy z tej dobrej atmosfery, póki trwa.

Jak państwo wiecie, jeszcze nie dokonaliśmy wyboru Prezydium Sejmu.

Dlatego przechodzimy do kolejnego punktu. Teraz poproszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego w trybie art. 162 ust. 1 Konstytucji RP. Panie Prezydencie! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Drodzy Rodacy! Jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, rządów Zjednoczonej Prawicy, to powiedziałbym tak: nie ma wolności bez godności. Nie ma wolności bez godności, nie ma wolności bez wiarygodności, bo to właśnie dotrzymywanie słowa, wiarygodność przełożyły się na to, że dzisiaj godniejsze jest życie polskich rodzin, godniejsza jest praca, płaca, godniejszy jest - można tak też powiedzieć - stan finansów publicznych, godniejsza jest nasza polityka historyczna, godniejsza jest nasza polityka międzynarodowa. Pani Marszałek! Panie Prezydencie!

Stało się bardzo wiele dobrego na bardzo wielu polach. Zacznę od tego, co bardzo często jest przedmiotem debaty, przedmiotem dyskusji w tej Izbie: demokracji, wolności, konstytucji, praworządności. Otóż przypomnę, że w ostatnich wyborach mieliśmy rekordową frekwencję, rekordowo niski odsetek osób głosujących w nieważny sposób, rekordowo szybko podane wyniki wyborów.

Kiedy demokracja ma się lepiej? Kiedy demokracja w lepszy sposób znajduje odzwierciedlenie w tej Izbie, w izbach sejmikowych? Kiedy jest minimalny, rekordowy w ciągu 30 lat odsetek głosów nieważnych i jednocześnie rekordowa liczba głosów ważnych, [[Oklaski]] bo wyższa nawet niż w 1989 r. - nie procentowo, ale w liczbach bezwzględnych. Te 18,5 mln świadczy o tym, że demokracja ma się tak dobrze, mogę powiedzieć, jak nigdy wcześniej.

Przez te 4 lata działo się tutaj bardzo, bardzo wiele.

Polaków powiedziało, że wierzy w to, że ich dzieci będą żyły w lepszych warunkach niż oni sami. I to był piąty wynik na świecie i pierwszy wynik w Europie, pierwszy wynik wśród wszystkich państw rozwiniętych. Co się takiego stało w ciągu 4 lat, że z narodu pesymistów w 2015 r., w podobnych badaniach, zamieniliśmy się w naród optymistów? To retoryczne pytanie, ale działo się bardzo wiele. Działo się bardzo wiele w obszarze chociażby budowy miejsc pracy. Miejsc pracy utworzonych zostało tak wiele, że dzisiaj na pytanie o to, czy czujesz się bezpiecznie na rynku pracy, prawie 60%, bo 58% odpowiada: tak, czuję się bezpiecznie. 4 lata temu było to 8%. To jest jedna z przyczyn zasadniczej zmiany podejścia również do państwa, również do demokracji.

Ta rewolucja godności jednocześnie została potwierdzona przez międzynarodowe instytucje. To także przełożyło się na wiarę w wolny rynek, system wielopartyjny.

Poprawiło się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Świadczy to o tym, że właśnie w czasach naszych rządów, przez poprzednie 4 lata mieliśmy do czynienia z rozkwitem wolności, z rozkwitem demokracji. Szanowni Państwo! Odnieśliśmy bardzo wiele sukcesów. Instytucje międzynarodowe takie jak Bank Światowy podkreślają wagę i sukces naszego nowego modelu gospodarczego, nowej polityki strukturalnej, nowej polityki przemysłowej. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalicza polską gospodarkę do 22 - i postępuje w tym rankingu w górę w hierarchii - gospodarek najwyżej rozwiniętych i największych gospodarek na świecie.

Była wynikiem wielu wysiłków wielu polityków, którzy wcześniej przed nami hołdowali takim wartościom, wartościom solidarnościowym, na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim, którego ideały wyznaczały naszą drogę. Ale również ta droga była skutkiem przygotowania wielu zmian, wielu zmian w gospodarce. Czasami wydaje się, że to, co jest blisko oczu, najbliżej naszych oczu, jest najbardziej oczywiste, ale zarazem często potrafimy to przeoczyć. Bo dzisiaj 500+ wydaje się projektem banalnym, banalnie prostym, oczywistym, ale przecież wiemy doskonale, w jakich okolicznościach był on wdrażany. Wiemy, jak wiele dobrego zrobił dla likwidacji ubóstwa, dla zmniejszenia nierówności, dla poprawy całej gospodarki, dla wyrównania szans, wielu szans milionów polskich rodzin. To działanie, któremu w dużym stopniu zawdzięczamy również nasze wielkie zwycięstwo, wielkie zwycięstwo 13 października, miesiąc temu. Patrząc na różne dziedziny życia, warto podkreślić, że także w tych, których reformowanie, zmiany muszą z natury rzeczy dotyczyć wielu kadencji, odnieśliśmy wiele sukcesów, np. w obszarach, które często przez przedsiębiorców są wskazywane jako problematyczne. Przedsiębiorcy nie lubią biurokracji, nie lubią ustaw, nie lubią zmian ustaw.

W czasach wcześniejszych średnio było to 25 do 30 tys. stron, teraz jest to 15 do 20 tys. stron, a więc ograniczyliśmy biurokrację. Przedsiębiorcy nie lubią kontroli skarbowych. W 2015 r. tych kontroli skarbowych było 35 tys. To są oficjalne dane. Chcę też w tym miejscu, szanowni państwo, podziękować w szczególny sposób naszym skarbowcom, Krajowej Administracji Skarbowej. bo ona dzisiaj podlega bardzo szczególnym atakom.

I dlatego chcę gorąco podziękować wszystkim skarbowcom z Krajowej Administracji Skarbowej. To wasze wielkie dzieło. Nie dajcie sobie wmówić, szanowni państwo, nie dajcie sobie wmówić, drodzy rodacy. W wielkiej organizacji - każdy, kto taką zarządzał, wie o tym doskonale - zawsze znajdzie się kilka czarnych owiec, kilka osób, które są nieuczciwe. Właśnie Biuro Informacji Wewnętrznej powołane w ramach Krajowej Administracji Skarbowej. Wielki wysiłek tej organizacji spowodował tę gigantyczną różnicę. Wysoka Izbo!

Ile jest teraz, w ostatnich latach?

Nie pracujcie na rzecz interesów różnych nieuczciwych przestępców.

Ale ja raz jeszcze chcę podziękować, pochwalić Krajową Administrację Skarbową za wspaniałe dzieło, za to, że państwo to zrobiliście, za to, że potrafiliście zastosować takie instrumenty, żeby podnieść nasz poziom, poziom jakości systemu podatkowego w Polsce do niebywałych, nierejestrowanych wcześniej wyżyn. Przy was ten legendarny Eliot Ness to właściwie gasnąca, blednąca gwiazda. Bardzo wam za to, wszyscy skarbowcy, dziękuję. Wysoka Izbo! Chciałbym też przejść do paru innych bardzo ważnych, kluczowych dziedzin naszego życia. Służba zdrowia. 4 lata, wielkie zmiany. Zacznijmy od tego, o czym każdy mówi w kontekście służby zdrowia. Wydatki na służbę zdrowia przez 4 lata wzrosły z 70 mld do To ponad 50%.

Kolejki również się skróciły po raz pierwszy. W innych przypadkach zatrzymaliśmy wzrost kolejek. Przejdę do innego obszaru: samorządy.

Przez poprzednie 8 lat było to 12 mld zł. Tyle więcej dostają samorządy z centralnego budżetu.

Kraków. W czasach Platformy Obywatelskiej wynosił ok. 22%. A więc to jest ta jakościowa różnica. Jak widzicie, posługuję się tylko nagimi faktami, twardymi danymi finansowymi, bo je najtrudniej jest kwestionować. Za chwilę można zajrzeć na strony samorządów, Ministerstwa Finansów i można je zweryfikować.

A więc wielka jakościowa zmiana. Reforma gimnazjów, którą obiecaliśmy i którą zrealizowaliśmy. To wielka zmiana, którą też trzeba podkreślić w kontekście oświaty. Szanowni Państwo!

spytajcie w tych województwach o wnioski: czy były jakieś odrzucone z powiatów i gmin. Takie wnioski, które były odrzucone, były w minionych latach. Teraz, w tym roku, na skutek wielkości naszego programu. Wielki nowy program rozwoju kolejnictwa w Polsce, odbudowa linii kolejowych między mniejszymi miastami. Kielce - Busko-Zdrój.

Panie premierze, przepraszam. Bardzo proszę. więc zmiany w kolejnictwie są zasadnicze.

Wcześniej, 4 lata temu, było to 296 miast. Szanowni Państwo! To jest znakomity postęp, to jest wielka zmiana. W ponad 100 miastach w Polsce będzie się zatrzymywał pociąg. To wielka zmiana na rzecz zmniejszenia wykluczenia dostępu mieszkańców do kolei. Szanowni państwo, Wysoka Izbo.

Pod nieobecność chciałbym podziękować pani premier Beacie Szydło. Dziękuję bardzo, pani premier. Dziękuję wszystkim ministrom i parlamentarzystom. Przez te 4 lata dokonaliśmy też wielkiej zmiany w polityce godnościowej, w polityce historycznej. Wiemy doskonale, jak ważna jest soft power. We współczesnym świecie ona jest czasami nie mniej ważna - ta miękka siła, która zależy od tego, jak nas postrzegają, czy potrafimy walczyć o prawdę historyczną - od twardych parametrów gospodarczych czy militarnych. I tutaj nastąpiły zasadnicze zmiany. Kiedy patrzę, sięgam myślami wstecz, patrzę na wspaniałe momenty, takie jak obchody stulecia odzyskania niepodległości. 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, wystąpienie prezydenta Niemiec. Zasadnicza zmiana w postrzeganiu Polski. Zasadnicza zmiana w postrzeganiu prawdy historycznej. To daje nam niesamowitą siłę, siłę na przyszłość, ponieważ od tego zależeć będzie w ogromnym stopniu również to, jak będziemy potrafili realizować nasze interesy w przyszłości, nasze interesy w Unii Europejskiej.

Zmierzam do końca.

Nigdy też nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Kończąc, chcę powiedzieć tak. rzadko kiedy odchodzący rząd może powiedzieć tak: Skarbiec jest w dobrym stanie. Ludzie mają pracę. Granice są bezpieczne. Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość. Jeszcze chwileczkę, bardzo proszę o spokój. Myślę, że możecie państwo sobie na to pozwolić. Szanowni Państwo! Chcę na koniec podzielić się z państwem taką osobistą refleksją. Równo 4 lata temu. marszałek senior poprzedniej kadencji. Zapytał, czy będziemy w stanie zmniejszyć obszary biedy, czy ambitnym ludziom damy szansę realizować ich aspiracje, ich talenty, czy zapewnimy, że bohaterowie „Solidarności” będą uczczeni. Że dzisiaj, po tych 4 latach, na pewno jeszcze nie wszystko, ale bardzo wiele zrobiliśmy. Uczyniliśmy bardzo dużo, żeby Polska była lepsza. Dlatego w ślad za słowami Stanisława Thugutta z PSL „Wyzwolenie”, który powiedział: „Idziemy w daleką drogę, nie dotrzemy tam, gdzie jest kres tej drogi, bo idziemy w pewnej sztafecie. Jeżeli niektórzy z nas nie dotrą. to będziemy ciepło tych ludzi wspominać, ale my musimy iść dalej” I ja, szanowni państwo, też chcę tak podsumować. Jesteśmy w pewnej sztafecie, chcemy iść dalej. Chcemy iść dalej ku lepszej, sprawiedliwszej Polsce. Dziękuję, panie premierze.

Proszę państwa, chciałabym zwrócić się z ogromną prośbą do państwa. Wtedy, kiedy przemawiał pan premier, i wtedy, kiedy miał swój czas, naprawdę niepotrzebne były komentarze z ław sejmowych, bo źle się mówi, kiedy inni przeszkadzają. Jeśli ktoś z państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę zapisać się do głosu, ale naprawdę trudno jest się skoncentrować na mówieniu wtedy, kiedy inni komentują głośno z ław. Bardzo państwa proszę o to, żeby tego nie robić. A teraz, proszę państwa, za chwileczkę ogłoszę przerwę. Ale panie pośle, to jest przerwa, która wynika z rozdziału 1 regulaminu Sejmu, który porządkuje dzisiejszy dzień przed Prezydium Sejmu. Za chwilę ogłoszę przerwę, w której oczekuję na przedłożenie projektu uchwały, o której mowa w art. 5 ust. 2 regulaminu Sejmu, dotyczącej ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu.

Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Poselskie projekty uchwał w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1 i 2) Sejm, zgodnie z art. 5 ust. 2 regulaminu Sejmu, ustala liczbę wicemarszałków w drodze uchwały. Na podstawie art. 5 ust. 4 regulaminu Sejmu do tego projektu uchwały nie stosuje się przepisów o terminie wniesienia i doręczenia projektów. Projekt tej uchwały rozpatruje się w jednym czytaniu. Proszę pana posła Łukasza Schreibera o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały z druku nr 1. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt i honor w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić projekt uchwały o liczbie wicemarszałków Sejmu.

Dziękuję panu posłowi. Proszę bardzo.

A w jakiej sprawie, panie pośle?

Z wnioskiem formalnym pan poseł Janusz Korwin-Mikke. Wysoki Sejmie! Z laudacji pani marszałek dowiedzieliśmy się, że ona żelazną ręką poprowadzi Sejm, że zaprowadzi porządek dla nas wszystkich. Do tej pory pani marszałek nie zdołała odebrać głosu panu premierowi, który przekroczył czas, a teraz nie potrafiła odebrać go człowiekowi, który wykorzystał hymn narodowy w celach partyjnych. Dziękuję, panie pośle. Proszę pana posła Krzysztofa Gawkowskiego o przedstawienie kandydatury pana posła Włodzimierza Czarzastego. Proszę. Wysoka Izbo! Od kiedy mi wiadomo, to hymn państwowy nigdy nie był partyjny. Jest państwowy. To tak dla przypomnienia. Szanowni Państwo! Mam wielką przyjemność zgłosić na funkcję wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i który w swojej pracy zawodowej i społecznej przez wiele lat był związany z kulturą. Jest przedsiębiorcą, wydawcą, założycielem jednego z największych polskich wydawnictw literackich - wydawnictwa Muza.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji wybrany z okręgu Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Jaworzna. Szanowni Państwo! Włodzimierz Czarzasty to osoba, która swoją pracą i zaangażowaniem udowodniła, że lewica dzięki determinacji wielu osób, ale skupionej w rękach lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej, może wrócić do Sejmu. Porozumienie lewicy to osiągnięcie, które dało nam szansę, żebyśmy mogli reprezentować tych wszystkich wyborców, którzy w liczbie ponad 2300 tys. nas wybrali i którzy dają nam szansę, żebyśmy dzisiaj mogli mówić o konstytucji, porozumieniu i współpracy. Włodzimierz Czarzasty był jednym z ojców tego porozumienia, współpracy i tak postrzega swoją misję w polskim parlamencie. Dziękuję, panie pośle. Proszę panią poseł Joannę Borowiak o przedstawienie kandydatury pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić rekomendację, kandydaturę pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej na funkcję wicemarszałka Sejmu. Pani poseł Małgorzata Gosiewska to działaczka społeczna, samorządowiec i parlamentarzystka. Dała się poznać jako osoba aktywna i nieobojętna na ludzką krzywdę. W młodości była związana z gdańskim Niezależnym Zrzeszeniem Studentów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Zawsze blisko mieszkańców, z misją pomocy najbardziej potrzebującym. Od początku politycznie związana z Porozumieniem Centrum. Członek założyciel Prawa i Sprawiedliwości. W Kancelarii Prezydenta pomysłodawczyni systemowej polskiej pomocy humanitarnej w rejonach konfliktów zbrojnych, w tym spektakularnych projektów socjalnych. Organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla poszkodowanych w wojnie dzieci gruzińskich, a także dla młodych Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Inicjatorka pomocy bezpośredniej - konwojów humanitarnych do zniszczonych miejscowości tzw. strefy buforowej w Gruzji czy też dla mieszkańców dotkniętego katastrofalnym trzęsieniem ziemi Haiti. Nigdy nie zapomniała o potrzebujących polskich dzieciach. Po tragicznym pożarze w Kamieniu Pomorskim zaangażowana w zorganizowanie wakacji dla dzieci pogorzelców, a także dla dzieci powodzian z Małopolski. Wsparcie Polski i pracę Małgorzaty Marii Gosiewskiej doceniły władze gruzińskie, honorując ją za działalność humanitarną Medalem Honoru i tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tbilisi. W działalności parlamentarnej skupiona przede wszystkim na obronie polskiej racji stanu i prawdy historycznej. Aktywna i obecna na kijowskim Majdanie podczas rewolucji godności, później wielokrotnie na pierwszej linii konfliktu ukraińsko-rosyjskiego w Donbasie. Autorka wstrząsającego raportu o rosyjskich zbrodniach wojennych na wschodniej Ukrainie - dokumentu złożonego w Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze jako dowód przestępczej działalności separatystów i ich rosyjskich mocodawców. Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP do czerwca 2019 r. Wiceprzewodnicząca zgromadzeń parlamentarnych Polski i Ukrainy oraz przewodnicząca zgromadzeń parlamentarnych Polski i Litwy. Przewodnicząca parlamentarnych grup dwustronnych Polski i Gruzji oraz Polski i Rumunii. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Bogate doświadczenie zawodowe i parlamentarne oraz wybitne zdolności organizacyjne dowodzą, że pani Małgorzata Maria Gosiewska jest właściwym kandydatem na funkcję wicemarszałka Sejmu IX kadencji.

Pani Marszałek!

Wierzę, że Senat będzie nas inspirował do dobrych rozmów, dobrej pracy, zaufania i wzajemnych rzetelnych, podmiotowych relacji. Ale mówię o tym w kontekście wyboru Prezydium Sejmu.

Bo wszyscy posłowie są równi: i ci z większości rządzącej, i ci z opozycji. Właśnie po to jest Prezydium Sejmu, po to jest marszałek, który ma tak duży mandat i jest drugą osobą w państwie, żeby gwarantować prawa opozycji, żeby prowadzić rzetelnie debatę, żeby być sprawiedliwym, uczciwym i przyzwoitym. Pani marszałek Kidawa-Błońska spełnia wszystkie te oczekiwania i posiada cechy, które prawdziwy, dobry marszałek czy wicemarszałek powinien posiadać. Od 2002 r. w samorządzie warszawskim, od 2005 r. w polskim parlamencie w różnych miejscach, ale zawsze tych najważniejszych: w komisji kultury, komisji etyki, wreszcie w Prezydium Sejmu. Była wicemarszałkiem, była także marszałkiem Sejmu.

To jest osoba najlepsza z możliwych na ważne miejsce. Jestem przekonany, że jej doświadczenie, ale też charakter, dobre emocje spowodują, że Prezydium Sejmu będzie pracowało lepiej i że tak jak wszyscy tutaj siedzimy, nie będziemy czuli różnicy, czy ktoś, kto reprezentuje Prezydium, jest z większości rządzącej, czy z opozycji, bo tak samo traktuje wszystkich posłów. Wszystkiego dobrego, bo uważam, że te wybory są ważne, bo one muszą gwarantować nam dobry, sensowny wybór i dawać gwarancję rzetelnej pracy Prezydium Sejmu, wicemarszałków, a także marszałka Sejmu. Dziękuję panu posłowi. Proszę panią poseł Lidię Burzyńską o przedstawienie kandydatury pana posła Ryszarda Terleckiego.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość kandydaturę na urząd wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana posła Ryszarda Terleckiego. Absolwent studiów historycznych, uczestnik działań opozycji antykomunistycznej i „Solidarności” Profesor doktor habilitowany, wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Żonaty, ma troje dorosłych dzieci. Od 2001 r. należał do pierwszych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, w którym kierował Biurem Edukacji Publicznej w Krakowie, a po wyborze Janusza Kurtyki na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej objął funkcję dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Pan poseł Ryszard Terlecki jest autorem kilkunastu książek. W roku 2006 jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Od 2007 r. poseł Prawa i Sprawiedliwości. W 2010 r. powołany do Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Od 10 listopada 2015 r. przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Funkcję wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pełni od 12 listopada 2015 r. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Bogate doświadczenie zawodowe oraz wybitne zdolności organizacyjne, o czym mieliśmy okazję się przekonać, wskazują, że pan poseł Ryszard Terlecki jest dobrym kandydatem na wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Proszę pana posła Władysława Kosiniaka-Kamysza o przedstawienie kandydatury pana posła Piotra Zgorzelskiego. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz’15 mam zaszczyt i przyjemność przedstawić kandydaturę posła Piotra Zgorzelskiego na funkcję wicemarszałka Sejmu IX kadencji.

Ukończył historię na wydziale historii Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, Uniwersytecie Warszawskim. Przez 15 lat był nauczycielem i dyrektorem szkoły w Leszczynie Szlacheckim. Przeszedł wszystkie szczeble samorządności. Pełnił funkcję wicewójta w gminie Bielsk w powiecie płockim, był starostą płockim, dyrektorem delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Trzykrotnie uzyskał poparcie społeczne w wyborach, a najlepszym świadectwem akceptacji społecznej dla Piotra Zgorzelskiego było podwajanie jego wyników wyborczych w każdych kolejnych wyborach. Każde kolejne wybory to dwa razy lepszy wynik uzyskany przez Piotra Zgorzelskiego. W latach 80. działał w Konfederacji Polski Niepodległej. Od ponad 30 lat jest związany z ruchem ludowym. Dzisiaj pełni funkcję sekretarza Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest współautorem Koalicji Polskiej, który przez ostatnie lata nie tylko w pracy parlamentarnej, ale również w pracy społecznej wykazał się swoimi zaletami i umiejętnościami. Jest osobą niezwykle skrupulatną, punktualną, mającą twardą rękę, o której była już dzisiaj mowa, i taka twarda ręka w Prezydium Sejmu jest potrzebna. Ale cechuje go też serdeczność i szlachetność wobec wszystkich parlamentarzystów, niezależnie od tego, z jakiej opcji politycznej pochodzą, wobec wszystkich, którzy pracują w Wysokiej Izbie, wszystkich pracowników Sejmu, Kancelarii Sejmu. Jest osobą, która gwarantuje bezstronność prowadzenia obrad, szacunek dla regulaminu Sejmu, szacunek dla wszystkich wartości związanych z demokratycznym państwem prawa, przestrzeganie reguł tego państwa oraz życzliwość wobec drugiego człowieka.

Dziękuję, panie pośle. Proponuję, aby w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego Sejm wysłuchał 3-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Głos ma poseł Borys Budka. Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wielce Czcigodna Wysoka Izbo! Szczęść Boże! Dobry Wieczór! Szczęść Boże w ciężkiej pracy dla ojczyzny! Po tym pokazie hipokryzji, jakim były przemówienia inaugurujące pracę Wysokiej Izby. mamy pokaz arogancji, jakim jest procedowanie tego składu Prezydium. Przybiera ono charakter dyktatu silniejszego, porozumienia ponad podziałami. To będzie popisowe Prezydium. Z przystawkami, rzecz jasna, z przystawkami. Koło Konfederacji, baczcie państwo, weszło do tego Sejmu jednakowoż z wyboru, z wyboru.

i dobrym obyczajem tej Izby w poprzednich kadencjach było włączanie do składu Prezydium Sejmu. którym przypada w udziale zaszczyt zasiadania w Konwencie Seniorów. To, że ta zasada została naruszona w minionej kadencji, to z różnych względów nie dziwi, tak jak też nie dziwi to, że ta kadencja dobiegła końca w składzie niekonstytucyjnym, ponieważ czcigodna pani marszałek zapomniała zawiadomić posła Kawęckiego o tym, że przypada mu w udziale zaszczyt zajęcia miejsca po śp. ministrze. Notabene nie wiem, co z tym fantem zrobi pani marszałek, bo przecież jest poseł, ale ślubowania odeń nie przyjęto. a Sejm obradował w niekonstytucyjnym składzie 459 posłów. A zatem ten dyktat silniejszego nie będzie przyjęty przez koło Konfederacji, które odda głosy przeciwko wicemarszałkom w tym składzie, tak jak głosowaliśmy przeciwko czcigodnej pani marszałek Witek. Nie pomyliliśmy się, problemy z uciszeniem niesubordynowanego posła były złym prognostykiem dla tej kadencji. Koło Konfederacji głosuje przeciwko, licząc na to, że w miarę rozwoju coraz ciekawszej sytuacji wy, szanowni państwo, którzy być może dzisiaj weźmiecie udział w tym podziale łupów, doznacie tegoż dyktatu na własnej skórze ze strony Prezydium swoich partii i wtedy.

Zamykam dyskusję. Informuję, że liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie wicemarszałków ustalonej w uchwale Sejmu, w związku z tym Sejm przeprowadzi głosowanie w tej sprawie kolejno nad poszczególnymi kandydaturami za pomocą urządzenia do liczenia głosów, stosując sekwencję pytań: kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.

Kto się wstrzymał?

Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pani poseł Małgorzaty Gosiewskiej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm bezwzględną większością głosów wybrał panią poseł Małgorzatę Gosiewską na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pani poseł Małgorzaty Kidawa-Błońskiej, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pana posła Ryszarda Terleckiego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Ryszarda Terleckiego na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Kto z pań i panów posłów jest za wyborem na stanowisko wicemarszałka Sejmu pana posła Piotra Zgorzelskiego, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Głosowało 450 posłów. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana posła Piotra Zgorzelskiego na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie punktów porządku dziennego w dniu dzisiejszym. Za chwilę zarządzę przerwę w obradach, podczas której zwołam posiedzenie Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów w sprawie kontynuacji 1. posiedzenia Sejmu oraz realizacji planowanego porządku dziennego. Zarządzam przerwę w posiedzeniu.